Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Pamiętam, jak w VIII kadencji powstawały Wojska Obrony Terytorialnej i z jakim niezwykłym atakiem ze strony totalnej opozycji spotkała się próba utworzenia tych wojsk. Wojska zostały powołane, funkcjonują, powstają kolejne jednostki. To oczywiście bardzo cieszy Polaków. Dlaczego? Dlatego że w bardzo krótkim czasie doszło do zweryfikowania tej decyzji.

Doszło do podtopień, doszło do małych huraganów. Okazało się wtedy, że Wojska Obrony Terytorialnej stanęły na wysokości zadania. Jako pierwsze ruszyły na pomoc ludziom, aby ratować mienie, ratować zdrowie i życie Polaków. Kolejna próba, z jaką dzisiaj spotykają się Polacy, to kwestie związane z epidemią.

To właśnie jako pierwsi żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej stawili się w domach pomocy społecznej, aby wspierać pracowników, a nawet przejmować opiekę nad pacjentami w chwili, kiedy personel uległ zakażeniu i nie mógł sprawować (Dzwonek) nad nimi opieki. W związku z tym mam pytanie do pana ministra: W jaki sposób. Pani poseł, czas. do tego, aby właśnie wspierać Polskę i Polaków w walce z epidemią? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie ministrze. Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Szanowna Pani Poseł! Wysoki Sejmie! Rząd polski od samego początku pandemii podejmował zdecydowane działania po to, aby ograniczyć skalę zachorowań i zapewnić bezpieczeństwo Polakom. Od pierwszych dni w te działania byli zaangażowani żołnierze Wojska Polskiego. W pierwszych dniach epidemii zdecydowałem, by działanie Wojska Polskiego zostało podzielone na dwie operacje: „Tarcza”, za którą odpowiadało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, i „Odporna wiosna” oraz później „Trwała odporność” realizowane przez Wojska Obrony Terytorialnej. Ta operacja jest wciąż realizowana. Wojska operacyjne wspierały Straż Graniczną oraz Policję. Żołnierze wspólnie z pogranicznikami zapewniali bezpieczeństwo na przejściach granicznych aż do momentu, kiedy granice zostały ponownie otwarte. Terytorialsi zajęli się m.in. pomaganiem instytucjom państwowym, samorządom czy szpitalom. Obecnie każdego dnia ok. 10 tys. żołnierzy walczy z pandemią, a kolejne 10 tys. jest w stałej gotowości do podjęcia działań. Cały czas żołnierze Wojska Polskiego zaangażowani są w budowę szpitali tymczasowych. Wojsko wsparło budowę 17 takich placówek na terenie całego kraju, m.in. w Lublinie, Rzeszowie czy Krakowie, oraz przygotowało samodzielnie dwa szpitale kontenerowe na warszawskim Bemowie i we Wrocławiu. Podjąłem także decyzję, aby wojsko zorganizowało szpital tymczasowy na terenie 1. Bazy Lotnictwa Transportowego na Okęciu, gdzie opiekę w razie potrzeby zapewnimy 250 pacjentom. Zbudowaliśmy już ponad 50 izolatoriów oraz ponad 20 polowych izb przyjęć. Przy Wojskowym Instytucie Medycznym na ul. Szaserów w Warszawie powstaje szpital halowy na potrzeby osób zakażonych koronawirusem. Cały czas żołnierze Wojska Polskiego podejmują działania, by odciążyć cywilną służbę zdrowia i pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych. Wspieramy prawie 700 szpitali i 173 stacje sanitarno-epidemiologiczne. Zdecydowałem także o włączeniu podchorążych z wojskowych uczelni w walkę ze skutkami epidemii. Podchorążowie Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w większym zakresie niż jeszcze kilka miesięcy temu wspierają dziś lekarzy i pielęgniarki. Wsparcie wojska otrzymało także 21 regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Żołnierze zaangażowani są m.in. przy preselekcji dawców krwi i osocza, przeprowadzają wywiady epidemiologiczne. Sami również organizują akcje krwiodawstwa i oddają osocze. Od marca żołnierze Wojska Polskiego oddali ponad 11 tys. l krwi, a 200 żołnierzy oddało osocze. Nie sposób nie wspomnieć o olbrzymim wysiłku, jaki każdego dnia wkładają żołnierze, aby usprawnić system pobierania materiałów do badań na obecność koronawirusa. Dziś Wojsko Polskie pobiera wymazy w ok. 300 punktach przyszpitalnych, działa także ponad 300 mobilnych zespołów.

Od początku pandemii wspieramy osoby samotne, starsze i pozostające w izolacji w domach z powodu koronawirusa. Łącznie jest to prawie 11 tys. kombatantów, seniorów i innych potrzebujących. Terytorialsi, żołnierze wojsk operacyjnych oraz podchorążowie dostarczają im pożywienie, leki i materiały pierwszej potrzeby. Opieką od pierwszych dni objęliśmy zarówno pensjonariuszy, jak i personel domów pomocy społecznej.

Żołnierze prowadzili ewakuacje, dezynfekcje, cały czas wspierają personel w opiece nad pensjonariuszami. Wielki wysiłek w przeciwdziałanie skutkom epidemii wkładają także wojska chemiczne. Nasze zespoły 7 dni w tygodniu dezynfekują szpitale, domy pomocy społecznej czy karetki. Wysoki Sejmie! Codziennie ponad 2,5 tys. wojskowych medyków, pielęgniarek i ratowników medycznych dba o zdrowie chorych i ratuje życie pacjentów. Cały czas pracuje 14 wojskowych szpitali, 5 ośrodków medycyny prewencyjnej oraz Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii. W szpitalach wojskowych 35% łóżek przeznaczonych zostało dla pacjentów zarażonych koronawirusem, siedem wojskowych laboratoriów cały czas wykonuje testy na obecność koronawirusa. Zdecydowałem, aby przeprowadzić obowiązkowe szkolenia medyczne (Dzwonek) dla żołnierzy Wojska Polskiego. W teoretyczno-praktycznych zajęciach dotyczących COVID-19, posługiwania się indywidualnymi środkami ochrony osobistej, a także udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w środowisku niebezpiecznym wzięli udział prawie wszyscy żołnierze. W razie potrzeby będą oni mogli nawet zastąpić personel medyczny przy realizacji niektórych zadań. W przyszłym roku takie szkolenia przejdą także żołnierze rezerwy. W drugiej połowie 2020 r. żołnierze przeszli kursy opieki nad pacjentem leżącym, dzięki czemu są lepiej przygotowani do wykonywania zadań opiekuńczo-pielęgnacyjnych, m.in. na rzecz osób starszych. Dziękuję bardzo. Z pytaniem dodatkowym, bardzo proszę, pani poseł Agnieszka Górska. Szanowni Państwo! Sytuacja związana z pandemią COVID w Polsce jest wciąż bardzo poważna i myślę, że do nas wszystkich dochodzą informacje o możliwości natężenia tej epidemii, powrotu. czyli tzw. trzeciej fali, tak.

Pan minister oczywiście już udzielił tej informacji, ale mnie interesuje jeszcze sytuacja dotycząca szczepień, albowiem te dwie sytuacje mogą zaistnieć w jednym czasie.

Dziękuję. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Oczywiście tak. Z inicjatywy Wojsk Obrony Terytorialnej np. zorganizowano bezpłatną infolinię, za pomocą której wsparcia osobom w kryzysie udzielali psychologowie WOT oraz wojsk operacyjnych. W listopadzie terytorialsi uruchomili całodobową infolinię wsparcia dla ośrodków pomocy społecznej organizacji pozarządowych, a bardzo chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Izby na akcję, którą rozpoczęliśmy 8 grudnia. Otóż właśnie wówczas, 8 grudnia rozpoczęliśmy kolejną akcję „Łączymy na święta”, skierowaną do osób chorych na COVID, pacjentów onkologicznych i seniorów, dla których zorganizujemy połączenia wideo z rodzinami i bliskimi, niezwykle istotne i rzeczywiście psychicznie wzmacniające te osoby. Osoby, które są chore, które są samotne poprzez wideokonferencje mogą porozmawiać z rodziną. Bardzo szczytna akcja. Jestem wdzięczny inicjatorom, żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej za podjęcie takiej inicjatywy. Oczywiście tak jak pytały panie poseł, Wojsko Polskie będzie uczestniczyć w narodowym programie szczepień. Żołnierze będą odpowiedzialni m.in. za dystrybucję i logistykę szczepionek, a także będą tworzyć mobilne zespoły szczepień. 13 szpitali wojskowych zostało zakwalifikowanych do narodowego programu szczepień przeciwko wirusowi SARS COVID-19. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Wojsko Polskie będzie pomagać tak długo, jak długo będzie wymagała tego sytuacja. Tak jak do tej pory, wykorzystując nasze doświadczenie, będziemy wspierać przede wszystkim cywilną służbę zdrowia, transportować do szpitali środki ochrony osobistej, płyny dezynfekcyjne, potrzebny sprzęt. Aby zminimalizować skutki koronawirusa i zahamować jego rozprzestrzenianie się, będziemy wykorzystywać wojskową infrastrukturę medyczną i korzystać z doświadczonej wojskowej kadry medycznej. Nie pozostawimy bez opieki i wsparcia seniorów, kombatantów, osób samotnych. Chciałbym dziś podziękować wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego i pracownikom wojska za tytaniczną pracę, jaką wykonują każdego dnia. Żołnierze już udowodnili, że na ich pomoc zawsze można liczyć. Przez ostatnie miesiące pokazali, że są gotowi dostosować się do wszystkich okoliczności i wspierać praktycznie każdy obszar funkcjonowania państwa. Na ich pomoc będziemy mogli liczyć także w najbliższych miesiącach. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Kolejne pytanie przygotowane przez parlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości, posłów Jarosława Zielińskiego, Arkadiusza Czartoryskiego i Roberta Gontarza, w sprawie przygotowanego przez rząd zakresu wsparcia ze strony państwa dla średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w ramach „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” i „Krajowej strategii rozwoju regionalnego 2030”, kryteriów przyjętych do aktualizacji deliminacji miast powiększających dystans rozwojowy i wskaźników kwalifikacji miast na listę ośrodków wymagających dedykowanej pomocy, a także możliwości włączenia do tego programu miast, które w wyniku ostatniej reformy administracyjnej utraciły status miasta wojewódzkiego. Pytanie skierowane do ministra funduszy i polityki regionalnej. Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Rzeczywiście tytuł skomplikowany, ale sprawa bardzo ważna. Jedną z podstaw programu Prawa i Sprawiedliwości i realizowanej od 5 lat polityki rządu jest zasada zrównoważonego rozwoju kraju. W ramach tej polityki rząd przygotowuje kolejny ważny instrument, który ma być wdrażany w najbliższej perspektywie finansowej. Na podstawie analiz ekspertów z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ustaliło listę 139 średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które zostały zakwalifikowane do dedykowanego wsparcia ze strony państwa. Program ten jest dobrze skorelowany ze „Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” oraz „Krajową strategią rozwoju regionalnego 2030” Ze względu na znaczenie społeczno-gospodarcze i polityczne tego projektu oraz zainteresowanie nim ze strony samorządów i opinii publicznej uprzejmie proszę pana ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. Po pierwsze, jakie wskaźniki i kryteria stanowiły podstawę do ukształtowania tejże listy 139 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze i powiększających dystans rozwojowy, które są przewidziane do dedykowanego wsparcia ze strony państwa? Po drugie, jakie będą mechanizmy i jaki jest planowany zakres oraz jaka jest planowana wielkość pomocy dla tych ośrodków miejskich dla wzmocnienia ich funkcji społeczno-gospodarczych? I po trzecie, czy możliwe jest objęcie przygotowywanym programem wsparcia miast, które utraciły w wyniku ostatniej reformy administracyjnej status ośrodków wojewódzkich, a nie zostały zakwalifikowane na listę tych 139 miast, ustaloną na podstawie wspomnianych wyżej kryteriów i wskaźników? Spośród byłych miast wojewódzkich na tej liście nie znalazły się Bielsko-Biała, Częstochowa, Kalisz, Koszalin, Leszno, Piotrków Trybunalski, Płock, Siedlce, Skierniewice i Suwałki. Włączenie tych miast do programu wsparcia ze strony państwa, przeznaczonego dla ośrodków tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Dzwonek), stanowiłoby spełnienie niezrealizowanej dotychczas, a zapowiadanej od czasu reformy administracyjnej dokonanej przez rząd AWS-UW, a więc od ponad 20 lat, koncepcji rekompensaty rozwojowej w związku z utratą przez nie dotychczasowych funkcji administracyjnych i społeczno-gospodarczych. Bardzo proszę, panie ministrze, o odpowiedź na te pytania. Mam nadzieję, że na trzecie będzie odpowiedź pozytywna. Dziękuję bardzo, panie pośle. Proszę o udzielenie odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej ministra Waldemara Budę. Bardzo proszę, panie ministrze. Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję za to pytanie, bo to rzeczywiście jest temat niezmiernie istotny z punktu widzenia najbliższej perspektywy dotyczącej środków europejskich, której realizacja zbliża się nieuchronnie.

Oczywiście mamy kryteria, bo opinia była zamawiana, stawialiśmy pewne warunki.

Jeżeli chodzi o tę grupę, która została wyselekcjonowana na podstawie tych kryteriów, następne kryteria, które w drugim etapie były wzięte pod uwagę, to starość demograficzna, saldo migracji, wykształcenie ludności, poziom edukacji szkolnej, ubóstwo dochodowe, aktywność społeczna, dostępność do usług, zaawansowana przedsiębiorczość, zamożność samorządów, zamożność mieszkańców w przeliczeniu na mieszkańca i na wydatki na inwestycje, stopa bezrobocia, dostępność przestrzenna oraz poziom urbanizacji. A więc de facto wszystkie zagadnienia społeczne, które wpływają na ten ogólny kształt rozwoju tkanki miejskiej, zostały wzięte pod uwagę.

Ja tutaj nie widzę żadnego problemu, tylko wydaje mi się, że to jest na tyle wyczerpujące, że znalezienie innego kryterium będzie niezmiernie trudne, ale oczywiście jesteśmy tutaj otwarci.

Po pierwsze, w nadchodzącej perspektywie takie narzędzie, które miałoby służyć tym ośrodkom, to zintegrowane inwestycje terytorialne, tzw. ZIT. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, gdzie trwają prace nad przygotowaniem tych zintegrowanych inwestycji terytorialnych na poziomie samorządów województw.

My oczywiście w ramach kontraktów programowych będziemy wymagać od samorządów, żeby mocno wskazywać i stawiać na ZIT-y, tak żeby bardzo nisko schodzić z tymi potrzebami inwestycyjnymi, żeby je rzeczywiście identyfikować, oczywiście w jakimś stopniu, bo środki europejskie mają to do siebie, że mają swoje limity, również w jakiś sposób czynić zadość tym wszystkim oczekiwaniom, które w tych miastach będą się pojawiały. Były tu wskazane miasta, które akurat nie zakwalifikowały się. Pan minister wskazał tutaj Piotrków, Leszno, Koszalin, Suwałki, Siedlce.

To też jest nasz pomysł na to, aby odpowiadać na zapotrzebowanie tych miast. A więc na pewno będziemy starali się koncentrować na tych ośrodkach średnich i małych. Panu ministrowi bardzo to leży na sercu i z taką determinacją o to walczy. Mam nadzieję, że uda się pomóc tym ośrodkom, które pan minister wskazywał. Będziemy pracowali nad tymi rozwiązaniami. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie pośle.

Ja nie kwestionuję tych kryteriów, które przygotowała Polska Akademia Nauk, one oczywiście są logiczne, są obiektywne i te miasta są zakwalifikowane według właśnie tychże kryteriów, ale pytanie moje jest takie, czy drugim kryterium, które można by rozważać, nie mogłaby być ta historycznie niezałatwiona sprawa byłych miast wojewódzkich, które straciły status takich miast. Część z nich weszła do tego programu, część oczywiście to są dzisiaj ośrodki wojewódzkie nowych, większych województw, ale zostało 10 miast, które zostały tutaj pominięte.

Bardzo proszę o rozważenie tej sprawy. Oczywiście o innych mechanizmach także warto myśleć, dziękuję, że rząd właśnie myśli o tych innych mechanizmach wsparcia, również dla subregionalnych ośrodków, ale, panie ministrze, postulat proszę rozważyć, bo on jest ważny z powodów politycznych, historycznych i rozwojowych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, zapraszam. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! My pokazaliśmy pewną otwartość w tym zakresie, bo, tak jak mówię, pierwsza lista i opracowanie wskazywały 119 miast, dzisiaj jest 138 czy 139, w związku z tym aktualizacja tej listy pod kątem szerszego ujęcia również innych ośrodków jest jak najbardziej możliwa. Pytanie tylko, jakie cechy indywidualne, specyficzne konkretnych jednostek uwzględnić, żeby można było je na tę listę wprowadzić. Ale chciałem z całą stanowczością powiedzieć, że ta lista nie rozstrzyga o tym, kto będzie miał, a kto nie będzie miał tej pomocy.

Proszę zwrócić uwagę, jaka jest skala - 139 podmiotów, taka jest skala wielkości. Ta opinia i to opracowanie jakby wskazują problem, czyli pokazują: tak, te ośrodki wymagają wsparcia, one się degradują społecznie i gospodarczo i musimy na nich skoncentrować swoją uwagę.

Proszę mi wierzyć, że z całą determinacją będziemy do tego podchodzić. Mamy zupełnie inną filozofię niż nasi poprzednicy, dla których ten system polaryzacyjno-dyfuzyjny miał działać w ten sposób, że duże ośrodki miały emanować swoimi zaletami w postaci rozwoju gospodarczego i społecznego na mniejsze ośrodki, czyli niejako w takiej kolejności, że dobrobyt wielkich ośrodków miał w jakiś sposób wpływać też na te małe. Okazało się, że związek między jednym a drugim jest bardzo niewielki, że jest wręcz przeciwnie, bo powiększało to różnice rozwojowe między tymi jednostkami, zwiększało, budowało demograficznie duże jednostki w związku z tym, że te różnice były coraz większe, a w niewielkim stopniu wpływało na rozwój małych ośrodków. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Jest to pytanie przygotowane przez posłów Koalicji Obywatelskiej Jacka Protasa, Marka Sowę, Monikę Wielichowską, Piotra Adamowicza, Barbarę Nowacką i Agnieszkę Pomaską w sprawie politycznego rozdania środków z II edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, skierowane do prezesa Rady Ministrów. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! W ostatnich tygodniach wielu Polaków zastanawiało się, dlaczego Unia Europejska tak konsekwentnie chce powiązania środków europejskich z mechanizmem warunkowości, praworządności.

Niejasny cel przyznawania środków, brak transparentnej procedury rozpatrywania wniosków, konsekwentne odmawianie przyznania środków w miejscach, w których Polki i Polacy wyrażają swoje niezadowolenie z polityki rządu, stanowi jaskrawy przykład złego gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

Jak to wygląda na mieszkańca? Na Podkarpaciu - 212 zł na osobę, na Podlasiu - 154 zł na osobę, a już w Wielkopolsce - 76, [[Dzwonek]] w lubuskim - 83, w opolskim - 88.

Dziękuję bardzo. Z upoważnienia prezesa Rady Ministrów odpowiedzi udzieli minister - członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Bardzo proszę, panie ministrze.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zacznę od tego, że mówimy rzeczywiście o wielkim wsparciu dla samorządów. Mówimy o wsparciu dla samorządów na poziomie 12 mld zł, o bezprecedensowej pomocy, która popłynęła do polskich gmin, powiatów i województw. Mówimy o wsparciu, którego rząd nie miał obowiązku udzielać, którego rząd na taką skalę, nawet w przybliżonej skali nigdy nie udzielił za czasów naszych szanownych poprzedników. Mówimy o wsparciu, które jest potrzebne po to, by podtrzymywać inwestycje lokalne także w naszych małych ojczyznach. Druga sprawa.

Co łączy takie miejscowości: Szczecin, Łódź, Kraków, Warszawa, Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Gliwice, Białystok, Gdynia, Lublin, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Opole, Rzeszów? To 17 z 20 największych beneficjentów tego programu.

Pozwolę sobie tylko wymienić bardzo dużych beneficjentów tego programu w drugiej turze: miasto Bydgoszcz, miasto Koszalin, powiat rawicki, powiat nowomiejski, gmina Starachowice, miasto Rybnik, miasto Tychy, miasto Częstochowa, województwo pomorskie, województwo opolskie itd.

To, że odeszliśmy od tej fatalnej koncepcji, która została zaproponowana przez naszych poprzedników, od tego modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego rozwoju kraju na rzecz modelu zrównoważonego, i z tej drogi zejść nie zamierzamy. A jeżeli panowie, państwo twierdzicie, że takie są kryteria, to proszę, wskażcie, miejcie odwagę i powiedzcie, które z tych projektów są niepotrzebne, które z tych projektów, na które zostały przyznane środki, powinno się zabrać. Nie wiem, jak jest w skali całego kraju, teraz nie mam takiej liczby, ale mogę podać na przykładzie mojego województwa kujawsko-pomorskiego: było łącznie 600 projektów, 100 zostało pozytywnie ocenionych przez komisję, rekomendowanych. A więc jest siłą rzeczy naturalną sprawą, że nie każdy z nich mógł być rozpatrzony, bez względu na czyjąkolwiek wolę.

Taki konkurs, jakich się odbywa wiele i odbywało się zawsze przez całe lata wiele. Dziękuję bardzo. Pan poseł Marek Sowa z pytaniem dodatkowym. Bardzo proszę, panie pośle. Wysoka Izbo! Panie ministrze, mówimy wyłącznie o drugim naborze w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o partyjnym rozdaniu 4300 mln zł, które zabraliście samorządowcom, nowelizując ustawy podatkowe we wrześniu 2020 r. Podzieliliście ich pieniądze i - jestem przekonany - chcieliście wyróżnić swoich, dać kasę swoim i ukarać tych, którzy może mają zdolność do samodzielnego zdania, którzy może czasami są krytyczni wobec tej władzy. Ale nie ukaraliście tych samorządowców. Ukaraliście mieszkańców tych wspólnot, miliony Polek i Polaków. Jeśli pan minister tak mówi o zrównoważonym rozwoju, którzy wam jest bliski, to jak uzasadnić, że jeden dostaje na wszystko, na cztery projekty, drugi nie dostaje nic? Co pan powie? W czym gorsi są mieszkańcy Andrychowa od mieszkańców Wadowic? Takich przykładów możemy wam tutaj dawać setki. Po prostu chcieliście podzielić Polaków.

Bardzo proszę, panie ministrze.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Ja przedstawiałem środki, które są ujęte łącznie, łącznie z pierwszego i drugiego naboru. a będzie jeszcze trzeci nabór. Tak, proszę państwa. Tak naprawdę rozumiem, bo to wybrzmiało z pańskiej wypowiedzi, w czym jest zasadniczy problem.

Bo to przed chwilą pan powiedział, że z tego powodu są straty dla samorządów. Tak będziemy chcieli - proszę nie krzyczeć - będziemy chcieli. To jest celem rządu, w którym mam zaszczyt zasiadać, rządu premiera Mateusza Morawieckiego, by Polacy mogli się bogacić, by podatki były możliwie najniższe.

Tak np. jedno z miast: zadaszenie stoku narciarskiego - 200 mln zł. Faktycznie, skandal, że nie dostali. Kto inny chciał budować stadion hokejowy za pięćdziesiąt parę milionów, skocznie narciarskie, akademię golfa z 6-dołkowym polem golfowym, napowietrzne ścieżki ekologiczne z kolejką gondolową. No jasne, takich projektów, mniej lub bardziej absurdalnych, też było mnóstwo. Oczywiście nie udaje się spełnić takich oczekiwań, bo też nie taki był cel tego funduszu.

Dziękuję bardzo, panie ministrze. Przechodzimy do kolejnego pytania.

Pytanie skierowane jest do prezesa Rady Ministrów. Bardzo proszę panią poseł Monikę Falej o zadanie pytania. Nie słychać. Teraz słychać? Pani Marszałek! Panie Ministrze! W dobie pandemii wszystkie ręce na pokład. Samorządy borykają się przez to z ogromnymi problemami, w ich budżetach aż trzeszczy. Dlatego też rząd utworzył Fundusz Inicjatyw Lokalnych, tzw. FIL. To pomysł rządu na wsparcie samorządów i rekompensatę w tych trudnych czasach. 4,35 mld zł bezzwrotnego wsparcia ma być przeznaczone m.in. na realizację projektów infrastrukturalnych, edukacyjnych czy cyfryzację. Pieniądze, które pochodzą z funduszu COVID-19, są dzielone przez rząd. Przykładowo województwo pomorskie otrzyma ze środków drugiego etapu 237 mln zł, ale pieniędzy nie będzie dla Gdańska czy Gdyni. Na liście beneficjentów nie ma największych miast Warmii i Mazur - Olsztyna, Elbląga czy Ełku. Śmiem uważać, że w tym przypadku nie decydowały kryteria merytoryczne, ale polityka. Z kolei województwo podkarpackie otrzyma ponad 452 mln zł rozdysponowanych w tej części konkursowej. Na Podkarpaciu rządowe środki dostało 150 z ponad 500 zgłoszonych zadań. Nic dostaną: Rzeszów, Tarnobrzeg, Krosno, Mielec czy Przemyśl. Tam nie rządzi PiS. Pieniądze nie trafiły do największych miast, które są zdecydowanym motorem napędowym gospodarki w danym regionie. Tym samym brak finansowania opartego na rzetelnych kryteriach zagraża optymalnemu rozwojowi regionów. Pytam zatem i oczekuję jasnej odpowiedzi: Jakie są zasady przyznawania pieniędzy? Proszę podać merytoryczne kryteria decydujące o wysokości wsparcia. Czy instytucja zarządzająca funduszem przygotowała algorytm służący stworzeniu (Dzwonek) listy rankingowej wnioskodawców i kto był w składzie komisji przyznającej dofinansowanie oraz czy i gdzie samorządy mogą się odwołać? Dziękuję bardzo. Z upoważnienia prezesa Rady Ministrów odpowiedzi udzieli minister - członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Zapraszam, panie ministrze.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na wstępie chciałbym wyjaśnić, że nie byłem w żadnej komisji, ale odpowiadam, jakie były kryteria. Kryteria, które wynikają jasno z uchwały, zostały wskazane wprost w uchwale nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Komisja, oceniając wnioski, brała więc pod uwagę następujące wskazane w § 10 uchwały kryteria: realizację zasady zrównoważonego rozwoju, kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko, koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji, liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ, relacje kosztu planowanych inwestycji do prognozowanego efektu, wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ, wreszcie zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. I to jest precyzyjna odpowiedź na pytanie, której się pani poseł domagała. Co do protestów samorządowców, to widzieliśmy protest części. Zresztą protest był średnio rozsądny - to jest najbardziej delikatne określenie - związany z negocjacjami w Unii Europejskiej, które prowadził rząd, które prowadził pan premier, nawołujący do natychmiastowego podpisywania wszystkiego, co leży na stole.

Ale oczywiście wszystko można sobie wyobrazić, za wszystko można próbować zwalać winę na rząd, a nie na samego siebie. Przypominam, że jest to wsparcie bezprecedensowe, to nie jest żadne wsparcie na zadanie dla samorządu, które zostało zlecone, to jest wsparcie po to, byśmy te inwestycje lokalne mogli dźwignąć. Są próby zakłamywania rzeczywistości, podczas gdy - o tym także wspomnę - największe miasta korzystają z szeregu programów, które są niedostępne, jak państwo wiecie, dla mniejszych miejscowości, a i tak wśród beneficjentów tego programu, największych beneficjentów, to one są na czele.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Bardzo proszę, pani poseł. Pan minister powiedział, że to jest śmieszne, że to jest awantura polityczna. To ja tylko przypomnę słowa pana premiera, który tłumaczył, że chce pomóc najbiedniejszym regionom: Skończyliśmy z logiką Polski A, B, C. Polska ma się rozwijać równomiernie. To ja pytam: Jak równomiernie? Dlaczego w takim razie województwo warmińsko-mazurskie, które jest jednym z najuboższych regionów, znajduje się na końcu tej listy?

Dziękuję. O udzielenie odpowiedzi bardzo proszę pana ministra Łukasza Schreibera. Zapraszam, panie ministrze.

Wielce Szanowna Pani Marszałek! Przedstawione przez panią poseł informacje są z pewnością nieprawdziwe.

To jest średnia, szanowni państwo, w skali kraju. A więc nie można stwierdzić, że województwo warmińsko-mazurskie było w jakikolwiek sposób tutaj pokrzywdzone. Ma średnie wsparcie w skali kraju, tak jak to powiedziałem. Naprawdę, ja rozumiem, że każdy może próbować podawać przykłady ze swojego regionu, także miejscowości, które akurat w drugim naborze nie załapały się na środki, w ramach konkursu nie zostały im przyznane środki. Tak, takich miejscowości jest cały szereg w Polsce, ale to w żaden sposób nie uzasadnia państwa tez i bardzo bym prosił, aby o tym pamiętać. I naprawdę nie ma potrzeby mówienia mieszkańcom swoich regionów i przekazywania informacji, które są niezgodne z rzeczywistością. Mogę podawać szereg liczb, jak w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego, i mogę państwu powiedzieć z ręką na sercu, że przecież przytłaczająca większość tych środków trafiła do gmin, do powiatów, które nie mają nic wspólnego z obecną większością parlamentarną.

A trzecia tura jest przed nami i w trzeciej turze, jak rozumiem, kolejne samorządy uzyskają wsparcie. Tak że zachęcam do tego wszystkich samorządowców, wbrew tym krzykom, które mają miejsce tutaj, na sali, aby ubiegać się o te środki, aby składać pomysły w konkursach, aby proponować dobre rozwiązania, i niekoniecznie może za kilkaset milionów, ale takie, które są potrzebne mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o spokój. Kolejne pytanie przygotowane przez posłów Koalicji Polskiej Stefana Krajewskiego, Jana Łopatę, Dariusza Klimczaka, Mirosława Maliszewskiego i Marka Sawickiego w sprawie podziału środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych skierowane jest do prezesa Rady Ministrów. Pytanie zadaje pan poseł Jan Łopata. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pisemną formę pytania w sprawach bieżących otrzymał pan, otrzymaliście państwo od nas. Myślę, że nie będziemy go teraz powielali, tym bardziej że chyba sytuacja jest bezprecedensowa.

Bardzo bym pana prosił, by pan tego nie czynił. Bo program jako program jest i potrzebny, i warto, żeby był kontynuowany, chodzi tylko o pewne uszczegółowienie i chodzi o to, żeby był sprawiedliwy podział, a tak nie jest, co panu tutaj państwo posłowie do tej pory udowadniali. Przypominam tylko, panie ministrze, że łaskawie dzielicie środki, pieniądze publiczne, nie swoje, budżetowe, a może nawet z deficytu, i warto, by opinia publiczna nie miała w tej sprawie żadnych wątpliwości. Proszę również nie używać tej retoryki, że chcemy kogoś pozbawić pieniędzy, wskazać wniosek, który był niewłaściwy. To nie nasza rola, nie rola opozycji ani tych, którzy tych pieniędzy nie otrzymali. W to nie wchodzimy. Chociażby na pytaniu, czy z prac komisji odpowiedzialnej za ten podział sporządzono protokoły, czy są karty oceny tych wniosków. Ja dodatkowo zadaję panu pytanie o techniczną stronę. Nie liczyłem, ile tych wniosków z całego kraju jest, ale biorąc pod uwagę, że z lubelskiego jest 836, to było to parę tysięcy wniosków. Jak ta sześcio- czy siedmioosobowa komisja technicznie dokonywała tego wyłonienia? Gdzie są te protokoły, gdzie są te karty oceny? Dziękuję, panie pośle. Z upoważnienia prezesa Rady Ministrów odpowiedzi udzieli minister - członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Zapraszam, panie ministrze.

Wysoka Izbo! Jak już wspominałem, nie byłem członkiem tej komisji, nie jestem w stanie panu udzielić informacji w sprawie szczegółów technicznych, które wiążą się z tym, w jaki sposób podchodzono do tego i w jaki sposób sporządzano protokoły. Ale niewątpliwie, jeżeli wielce szanowny pan poseł zwróci się z takim pytaniem, a ono padło tutaj, to na pewno także odpowiedź będzie udzielona na piśmie, bo tak jak mówię, w tej chwili tego uczynić nie jestem w stanie. Mówienie o zbulwersowanej opozycji i zbulwersowanych samorządach, dobrze pan wie, jest mówieniem zdecydowanie na wyrost, bo jestem przekonany, że w sytuacji, w której wszyscy te środki otrzymali, w sytuacji, w której trzecia tura jest jeszcze przed nami, w sytuacji, w której.

Mamy 170 jednostek samorządu terytorialnego, a dziewięćdziesiąt kilka wniosków zostało zaopiniowanych pozytywnie, czyli siłą rzeczy nawet gdyby na jedną jednostkę samorządu terytorialnego przypadał jeden projekt, to nie każdy mógłby otrzymać wsparcie. A nie jest pan w stanie wykazać na tym przykładzie, że - rzekomo - widać tam partyjny klucz.

Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie ministrze. Panie Ministrze! Są dwa wnioski skierowane do NIK: Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Obywatelskiej.

A więc mam nadzieję, że pan minister te dzienniki zaskarży. 9-osobowa komisja dostała wnioski od wojewodów ze wskazaniem, kto może, a kto nie może, kto powinien, a kto nie powinien. I w tej 9-osobowej komisji są tak zacne nazwiska jak Krzysztof Kubów, szef gabinetu politycznego pana premiera, poseł i wiceminister Iwona Michałek oraz poseł i wiceminister Waldemar Buda.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie ministrze.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Bo taki sposób myślenia, taki sposób poczucia niesprawiedliwości jest często w tych województwach, w których rządzicie, i to rządzicie od lat. Gdybyście pojechali - zapraszam - np. do mojego województwa kujawsko-pomorskiego, to moglibyście posłuchać, co o różnych konkursach przygotowywanych przez waszych włodarzy myślą i mieszkańcy, i samorządowcy. Dziękuję bardzo. Obiecywał, proszę to wypełnić.

Pytanie jest przygotowane przez posłów Koalicji Obywatelskiej: Barbarę Nowacką, Monikę Rosę, Monikę Wielichowską, Klaudię Jachirę, Michała Szczerbę, Urszulę Zielińską, Katarzynę Lubnauer, Dariusza Jońskiego i Aleksandrę Gajewską i dotyczy prześladowań uczestniczek i uczestników protestów w sprawie praw kobiet oraz kosztów zabezpieczenia przez Policję i służby tych protestów w całym kraju, w szczególności pomników na placu Piłsudskiego oraz domu Jarosława Kaczyńskiego. Pytanie jest skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Bardzo proszę, pani poseł.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Od 22 października przez Polskę przetacza się fala protestów w obronie praw, godności i bezpieczeństwa kobiet. To są protesty pokojowe, protesty liczne i radosne, natomiast widzimy, w szczególności od połowy listopada, znaczną brutalizację ze strony władz, ze strony policji.

Barierki szpecą i utrudniają ruch właściwie w całym centrum Warszawy, do Sejmu dojść się nie da, i to nawet wtedy, kiedy protestów nie ma, do ochrony pomników, ochrony domu pana Kaczyńskiego wykorzystano kilka dni temu 80 radiowozów. W całej Polsce siły policji mobilizowane są do pilnowania, spisywania, działań przeciwko pokojowo protestującym w ramach obowiązujących przepisów prawa obywatelom.

Jakie są tego koszty? Czyje to są decyzje? Czy w pana ocenie jest to adekwatne do poziomu zagrożenia, jakie stanowią pokojowo protestujące kobiety i młodzież? Dziękuję, pani poseł. Odpowiedzi udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik. Zapraszam, panie ministrze. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym odnieść się do tego pytania w sposób jak najbardziej pełny i precyzyjny, ale na początku chciałbym sprostować pewną rzecz. Pani poseł raczyła powiedzieć, że są to pokojowe protesty w ramach przepisów prawa.

Te przepisy obowiązują, zostały uchwalone przez Wysoki Sejm i nie ma co do tego wątpliwości.

Wszystkie działania Policji podejmowane od 22 października to jej ustawowe zadania - także ochrona Sejmu, także ochrona obywateli, także ochrona protestujących, bo zdarzały się sytuacje, gdzie między jednymi a drugimi grupkami protestujących dochodziło do zwarć. Tam zawsze pojawiała się Policja, która rozdzielała protestujących i uspokajała sytuację.

Chciałbym podkreślić, pani poseł, że w związku z wykonywanymi w ostatnich miesiącach zadaniami Policja nie zwiększyła swojego budżetu, nie trzeba było zwiększać budżetu Policji. To wszystko było w ramach zaplanowanych na ten rok środków finansowych.

Muszę panią uspokoić, pani poseł, te osoby zostały ujęte przez Policję i staną przed sądem, żeby odpowiedzieć za swoje czyny.

Dzisiaj rano dwaj policjanci z komendy miejskiej w Tychach zostali zatrzymani przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Wszędzie tam, gdzie dojdzie do przekroczenia uprawnień, takie działania będą prowadzone.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Po pierwsze, konstytucja gwarantuje nam prawo do zgromadzeń - art. 57 konstytucji. Art. 31 konstytucji mówi, że ograniczenia praw i wolności mogą być stanowione jedynie w ustawie. Państwo zrobiliście to rozporządzeniem, nie wprowadziliście stanu nadzwyczajnego.

Dziękuję, pani poseł. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie pośle, pytanie padło, pada odpowiedź. Proszę o spokój. Wysoka Izbo! Chciałbym powiedzieć tak: Środki przymusu bezpośredniego są przewidziane przepisami prawa, ustawą i policja stosuje te środki przymusu bezpośredniego zgodnie z przepisami ustawy.

Powiem tak: Jako minister, jako wiceminister spraw wewnętrznych i administracji niestety ubolewam głęboko nad tą sytuacją. Przy używaniu środków przymusu niestety czasami może zdarzyć się taka sytuacja, że dojdzie właśnie do tego typu uszczerbków, i ubolewam nad tą sytuacją. Ta sytuacja jest wyjaśniana. Nie dalej niż wczoraj, wiedząc, że będę odpowiadał przed Wysoką Izbą, poprosiłem komendanta głównego Policji o przedstawienie mi tej sytuacji. Ta młoda dama, młoda pani będzie jeszcze przesłuchiwana w tym postępowaniu, jeżeli się stawi i będzie chciała złożyć zeznania, i jej zeznania będą ważnym elementem tego postępowania. W tej chwili, na tym etapie nie ma powodów do tego, żeby uważać, że policjanci użyli środków przymusu niezgodnie z przepisami. To była sytuacja blokady ulicy, ta pani siedziała na ulicy, ul. Wilczej, policjanci używali siły fizycznej. Chciałbym, żeby do niej nie doszło.

Natomiast to nie jest tak, że większość jest z 11 listopada.

Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie przygotowane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości: Andrzeja Gawrona, Lidię Burzyńską i Mariusza Trepkę, w sprawie wsparcia dla rolników prowadzących hodowlę świń w cyklu otwartym - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Mamy obecnie trudny czas pandemii, który dotyka wszystkich nas, ale też w dużym stopniu sektor rolniczy.

Aby zmniejszyć ryzyko trwałego wycofania się z produkcji, ministerstwo przygotowało program pomocowy w związku z kryzysem COVID-19.

Ostatnio pojawiły się informacje o tym, że również rolnicy, hodowcy w cyklu otwartym mogliby liczyć na taką pomoc. Prosiłbym pana ministra o szczegółowe wyjaśnienie, czy to będą podobne zasady jak dla producentów wieprzowiny w cyklu zamkniętym, czy jakieś nowe elementy tego programu, jakie są w ogóle zasady i do kiedy można składać wnioski.

Dziękuję bardzo. Odpowiedzi na to pytanie udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi minister Ryszard Bartosik. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie!

W tej chwili trwa nabór prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Taki rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w systemie informatycznym.

Wysokość pomocy ustalono na poziomie analogicznym do tego z rozporządzenia PROW, uznając, że projektowana pomoc jest komplementarna do pomocy udzielanej producentom świń w obiegu zamkniętym na podstawie rozporządzenia PROW. Producenci świń mogą składać wnioski o pomoc do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 20 grudnia. Założono, że proponowana pomoc może być kumulowana, łączona z pomocą udzielaną z tytułu prowadzenia innych niż produkcja świń w cyklu otwartym kierunków produkcji na podstawie rozporządzenia PROW.

Wnioski cały czas spływają. Na pomoc przeznaczono 175 mln zł. Ten import znacząco się nie zwiększa. Według danych głównego inspektora weterynarii sytuacja jest pod kontrolą i nie stwierdziliśmy nielegalnego importu. Jeśli import się odbywa, to zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Pytanie uzupełniające zada pan poseł Mariusz Trepka. Bardzo proszę. Wysoka Izbo!

Natomiast moje dodatkowe pytania są takie.

Dziękuję. Panie ministrze, proszę o udzielenie odpowiedzi. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Wynika to z tego, że wzorowaliśmy się na pomocy, która jest taka sama jak w rozporządzeniu

Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie przygotowane przez posłów Marka Rząsę, Tomasza Kostusia i Dorotę Niedzielę z Koalicji Obywatelskiej w sprawie braku wsparcia dla podkarpackich rolników poszkodowanych w wyniku długotrwałych ulewnych opadów i stanu wypłat odszkodowań suszowych oraz za likwidację stada z powodu ASF na terenie całej Polski. Pytanie skierowane jest do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Panie Ministrze! Przed każdymi kolejnymi wyborami politycy PiS prześcigali się w odwoływaniu do etosu polskiej wsi, deklarowali szacunek dla ciężkiej pracy rolników.

Jestem tu dziś, by upomnieć się o polskich rolników, których w tym roku wyjątkowo doświadczyły niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Jako przykład posłuży mi województwo podkarpackie, w którym komisje gminne oszacowały straty w 3348 gospodarstwach rolnych, a ich wysokość wyniosła 51 mln zł. Z treści pisma resortu skierowanego pod koniec listopada do wojewody podkarpackiego wynika, że rolnicy nie otrzymają żadnej pomocy. Proponuje im się natomiast preferencyjne kredyty, składanie wniosków o odroczenie lub rozłożenie na raty składek na KRUS, płatności z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz ulgi w podatku rolnym. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy resort jest w stanie jeszcze raz pochylić się nad losem polskich rolników. Proszę jasno zadeklarować, czy rząd PiS przywróci dla nich programy pomocowe oraz zapewni, że wszyscy polscy rolnicy, którzy ponieśli straty z powodu suszy i podtopień, będą mogli liczyć na realną pomoc państwa, czy też utrzyma swoje stanowisko, że PiS umywa ręce od problemów polskiej wsi i mówi rolnikom: bierzcie kredyty i radźcie sobie sami. Dziękuję bardzo. O udzielenie odpowiedzi proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ministra Ryszarda Bartosika. Bardzo proszę, panie ministrze. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jeśli chodzi o udzielanie pomocy, to akurat rząd Praw i Sprawiedliwości wykazał się dużą determinacją.

Przeznaczono na to ogromne środki w postaci miliardów złotych, które trafiły do polskich rolników w związku z wystąpieniem suszy. Te pieniądze były duże. Nigdy w historii takich pieniędzy rolnicy nie otrzymali ze względu na kataklizmy, jakie występowały, i zmiany przyrodnicze. Dotrzymywaliśmy swoich zobowiązań, które zostały zgłoszone podczas kampanii wyborczych, ale także w naszych programach. Reakcja na największą suszę od lat była ogromna. W porównaniu do rządów Platformy Obywatelskiej, można to udowodnić liczbami, ta pomoc była dużo, dużo większa. Natomiast jeśli chodzi o pismo, do którego pan poseł raczył się odnieść, by zarzucić nam, że proponujemy preferencyjne kredyty, chciałbym przypomnieć, że taka propozycja wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. Nie będę odnosił się do tego, kto wtedy sprawował władzę. My to utrzymujemy i nadal proponujemy tego typu wsparcie rolnikom. Korzystają z nich rolnicy na bazie rozporządzenia, które wydał rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Taka wówczas była pomoc, jeśli chodzi o wystąpienia gradobić, podtopień regionalnych, taka też obowiązuje teraz. Natomiast oprócz tej pomocy bezpośredniej, co chcę zauważyć, jest możliwość skorzystania ze środków, które zostały przeznaczone dla rolników w związku z wystąpieniem pandemii COVID. Kończy się drugi nabór. Ta pomoc rzeczywiście jest rozproszona, bo są kredyty i jest możliwość ubiegania się o pomoc z KRUS-u w związku z płaceniem składek.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski. Chcę też powiedzieć o innych środkach, które są przeznaczane na polską wieś, dla rodzin rolniczych. Dla przykładu w ostatnich dniach pan minister Grzegorz Puda uruchomił program, dzięki któremu rodziny rolnicze, dzieci z rodzin rolniczych otrzymają komputery.

Rzeczywiście regionalnej pomocy nie ma, opieramy się na funkcjonujących rozporządzeniach, które państwo raczyli przyjąć jeszcze w roku 2015. Tej pomocy jest wiele, ona jest rozproszona, ale rozproszona to nie znaczy, że mała. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie ministrze. Z pytaniem uzupełniającym pan poseł Tomasz Kostuś. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Mówił pan przez 5 minut, ale nie odpowiedział pan na proste pytanie zadane przez mojego przedmówcę. Pan poseł pytał, przypominam, czy w tym roku rolnicy otrzymają pomoc na zasadach, na jakich ją otrzymywali w roku ubiegłym. To jest proste pytanie, proste, panie ministrze. Natomiast wracając do kolejnej części naszych zgłoszonych pytań, panie ministrze: Ilu rolników w tym roku, i na jaką kwotę, nie otrzymało odszkodowań za likwidację stada z powodu ASF? Czy prawdą jest, że w ciągu ostatnich 5 lat z powierzchni Polski zniknęło ponad 120 tys. stad świń? Następne pytanie: Ile procent niewykorzystanych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trafi na pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19, wraz z wypłatą odszkodowań z tytułu suszy za rok 2019? I ostatnie pytanie: Ile środków wypłacono w formie odszkodowań z tytułu suszy za rok 2019, a ile jeszcze zostało do wypłaty, w rozbiciu na rolników i hektary? Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie pośle.

Zgodnie z danymi agencji restrukturyzacji na dzień 14 grudnia 2020 r. wpłynęło 787 wniosków o powyższą pomoc na kwotę 1675 tys. zł i wydano 776 decyzji na łączną kwotę 1634 tys. zł. Pomoc realizowana jest na bieżąco i jest przeznaczona dla producentów rolnych, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa wydanym ze względu na wystąpienie ASF u świń na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zaprzestali produkcji świń.

Na pozostałe pytania szczegółowe, a było ich dużo, odpowiem panu posłowi na piśmie.

Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, jest taki szczególny czas. W zeszłych latach były organizowane dla osób bezdomnych, dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji wspólne wigilie, były też inne formy pomocy, ale ten okres pandemii spowodował, że musimy się zastanowić nad innymi możliwościami wsparcia tych najbardziej potrzebujących, czyli seniorów, samotnych matek czy osób bezdomnych.

Mam takie pytania. Jak to w skali kraju będzie zorganizowane? I proszę o więcej szczegółów na ten temat, bo rzeczywiście w tym świątecznym okresie jest to bardzo ważny temat, żeby nie zostawić tych ludzi samych z tym problemem. Dodatkowo dopytam: Jakie organizacje biorą udział w tym Solidarnościowym Konwoju Wsparcia Seniorów? Bo to jest bardzo cenna inicjatywa w okresie pandemii COVID-19. Bardzo dziękuję. Dziękuję panom posłom. Odpowiedzi udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej minister Stanisław Szwed. Zapraszam, panie ministrze. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za to pytanie.

Dzięki tej akcji powstał też Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Osoby, które chcą pomagać osobom starszym w ramach wolontariatu, wypełniając specjalną ankietę, mogą się do tego programu zapisać.

To wsparcie może polegać na robieniu zakupów, na innych czynnościach, które są wymagane czy potrzebne dla tej osoby. Na dzisiaj ponad 18 tys. osób skorzystało z tego programu.

Tutaj duża rola zarówno gminnych, jak i miejskich ośrodków pomocy społecznej, bo na nich spada ciężar komunikowania się, wysyłania tych osób i sprawdzenia danego wolontariusza, żeby to była osoba pewna, żeby nie było jakichś kwestii, które czasami się zdarzają, jeśli chodzi o osoby starsze.

To jest program, który ma na celu, aby w okresie najbliższych dni, w okresie świątecznym wesprzeć najbardziej potrzebujących takiego wsparcia, osoby starsze, osoby bezdomne, bo tutaj był klucz do tego, od czego wychodziliśmy, czyli osoby bezdomne czy samotne matki.

Takich punktów będzie uruchomionych w skali kraju 12 i w ramach tych punktów wszystkie organizacje, które chcą w tym wziąć udział, muszą się zwrócić do Caritasu czy Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta i poprzez tę ścieżkę wykorzystywać możliwość udzielania pomocy. Przewidujemy, że w ramach tej pomocy materialnej, którą przekazuje Agencja Rezerw Materiałowych, będzie ok. 100 mln t żywności.

Wiemy też, że te organizacje mają dobre rozeznanie, jeśli chodzi o pomoc w danym terenie, w danej gminie. Myślę, że to jest bardzo dobry program, który pomoże osobom starszym w tym trudnym czasie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów to w aktualnym czasie pandemii pożyteczne wyzwanie, które podejmują premier, rząd i ministerstwo. Ja serdecznie dziękuję za tę jakże cenną inicjatywę. Na to bardzo konkretne pytanie ewentualnie poproszę o informację na piśmie. Dziękuję. Dziękuję, pani poseł. Pan minister Stanisław Szwed. Zapraszam do udzielenia odpowiedzi.

Ważne jest, żeby od tych organizacji organizacje pozarządowe też odbierały te środki i dostarczały do poszczególnych osób czy do poszczególnych organizacji, czy do schronisk, w zależności od sytuacji.

Przez to działanie będziemy mogli łatwiej dotrzeć z pomocą do osób, które tej pomocy potrzebują, szczególnie w okresie świątecznym.

Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Kolejne pytanie przygotowane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości Barbarę Bartuś, Arkadiusza Mularczyka i Jerzego Polaczka w sprawie postępów w realizacji budowy drogi krajowej nr 75 Brzesko - Nowy Sącz, tak zwanej... Sądeczanki. Jako pierwsza pytanie zadaje pani poseł Barbara Bartuś. Bardzo proszę, pani poseł. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Droga krajowa nr 75 to jedyna droga łącząca powiat nowosądecki z autostradą A4. Nowy Sącz to trzecie co do wielkości miasto województwa małopolskiego, przez które przebiega szlak drogowy do granicy ze Słowacją, a natężenie ruchu samochodowego, w tym pojazdów o wysokim tonażu, jest bardzo duże. Dlatego też mieszkańcy całego regionu, nie tylko regionu Sądecczyzny, ciągle dopytują i z wielką niecierpliwością oczekują wybudowania tzw. sądeczanki. Według założeń sądeczanka będzie dwujezdniową drogą przyspieszonego ruchu. Zainteresowanie jest bardzo duże i to nie tylko mieszkańców Sądecczyzny, ale też innych, bo tak jak powiedziałam, ta droga nie tylko ma dobiec do Nowego Sącza, ale to jest połączenie też z południem Europy. To zainteresowanie jest duże, ale dużo jest też fake newsów. W ostatnim okresie bardzo rozgorzała o tym dyskusja, jest obwiniany rząd Prawa i Sprawiedliwości: jeżeli rządziłaby Platforma Obywatelska, to już jeździlibyśmy tą sądeczanką, bo już była wpisana, bo już by była, a niestety ciągle są opóźnienia. Panie Ministrze! Proszę, żeby odpowiedział pan nam, ale przede wszystkim mieszkańcom, czy sądeczanka w ogóle była ujmowana w projektach poprzednio rządzących, czy ona była realnie wpisana. Jeszcze przed pana odpowiedzią bardzo prosiłbym o udzielenie informacji, czy.

Dziękuję panu posłowi. O udzielenie odpowiedzi proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury ministra Rafała Webera. Bardzo proszę, panie ministrze. Wysoka Izbo!

Sądeczanka jest niezmiernie ważna z punktu widzenia rozwoju komunikacyjnego, gospodarczego i turystycznego. Można jednym zdaniem powiedzieć, że bez wątpienia na budowie tej drogi zyska zarówno społeczeństwo ziemi sądeckiej, jak i wszyscy ci, którzy korzystają z niej, docierając z południowo-wschodniej części Małopolski. Różnimy się w tej sferze od rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, które potraktowały tę inwestycję czysto populistycznie, obiecując jej realizację przed wyborami w 2015 r., ale nie zapewniając dla niej finansowania. Na papierze można wszystko napisać, papier wszystko przyjmie, natomiast jeżeli nie ma zapewnionego finansowania na realizację danej inwestycji, to jej wykonać po prostu nie można, i taka sytuacja miała miejsce za czasów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przede wszystkim zabezpieczyliśmy na jej budowę środki finansowe.

To pokazuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Mateusza Morawieckiego, jest przygotowany i zdeterminowany, aby tę inwestycję wykonać. Umowa z wykonawcą studium korytarzowego i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego została zawarta we wrześniu 2016 r., a więc również za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. A teraz kilka zdań o tym, w którym miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o przygotowanie tej inwestycji. W ramach obecnie opracowywanego studium korytarzowego firma projektowa przygotowała cztery wstępne warianty przebiegu. W 2017 r. odbyło się 15 spotkań z mieszkańcami i samorządami w gminach, wpłynęło ponad 10 tys. głosów w sprawie korytarzy. Na podstawie wniosków i sugestii mieszkańców i samorządów przeanalizowano 26 wariantów przebiegu korytarzy, co wynosi 1800 km hipotetycznych dróg. Mieszkańcy i przedstawiciele władz samorządowych sprzeciwiali się przebiegowi nowej drogi w pobliżu nieruchomości, w których aktualnie zamieszkują. Ustępstwa projektanta wobec gmin i mieszkańców danej miejscowości skutkujące zmianą przebiegu drogi powodowały kolizje z oczekiwaniami mieszkańców gmin sąsiednich.

I to jest clou tego problemu, to jest clou toczących się prac nad wyznaczeniem przebiegu wariantu sądeczanki. 15 stycznia 2018 r. w siedzibie oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie odbyło się spotkanie z parlamentarzystami i samorządowcami, na którym zaprezentowane zostały dwa warianty, A i B, korytarzy przebiegu. Poszukiwano przebiegów, które umożliwią spełnienie parametrów technicznych, z uwzględnieniem terenów osuwiskowych oraz czynników społecznych. Podstawowym kryterium społecznym była minimalizacja wydłużeń budynków. Uwzględniano także wszelkie kolizje z terenami cennymi przyrodniczo. W wyniku analizy przebiegów 26 wariantów korytarzy wybrano dwa warianty do dalszych prac nad dokumentacją. Pan minister Andrzej Adamczyk wykazywał tutaj również bardzo dużą aktywność. W kolejnym okresie wykonywane były m.in. badania geologiczne, inwentaryzacja przyrodnicza, analizy ekonomiczne i społeczne, po wykonaniu których przygotowana zostanie dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. W 2019 r. odbyły się kolejne spotkania informacyjne. Po spotkaniach wykonawca przeprowadził analizę i opracował raport z odniesieniem do uwag i wniosków.

Szczególnie istotne były analizy geologiczne, z uwagi na trudny teren, a także hydrologiczne i hydrauliczne, które wymagane są przez Wody Polskie. Jeżeli pani marszałek pozwoli zakończyć sekwencję.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Wód Polskich, centrali generalnej oraz wójtowie i burmistrzowie miast i gmin, przez które prowadzone były warianty tras. W efekcie spośród wszystkich analizowanych wariantów wstępnie wskazano, że do dalszych prac najlepsze będą warianty wskazane w wystąpieniu wnioskodawców: wariant C - najkorzystniejszy technicznie, wariant A - alternatywny, samorządowy i wariant F - alternatywny, najkorzystniejszy pod względem środowiskowym.

Dziękuję, panie ministrze. Też chcę poinformować pana ministra, że w najbliższy poniedziałek w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie odbędzie się posiedzenie zespołu parlamentarnego w sprawie właśnie sądeczanki, kolei Podłęże - Piekiełko, z udziałem dyrektora. Tak że jeżeli pan minister ma czas, to oczywiście też zapraszamy. To dotyczy nie tylko ziemi sądeckiej, Sądecczyzny, ale także ziemi brzeskiej i całego subregionu małopolskiego. Wiemy, panie ministrze, że są te trzy warianty: wariant C jako najkorzystniejszy pod względem technicznym, wariant A jako wariant alternatywny, który uzyskał pozytywną ocenę samorządowców, i wariant F jako najkorzystniejszy ze względów środowiskowych. Czy mamy już harmonogram kolejnych etapów prac, ze wskazaniem przewidywanych terminów? Wiemy, że jest też zapewnione finansowanie. Pan minister mówił też o czwartym wariancie. Jakby pan mógł to przybliżyć. Dobrze, dziękuję bardzo. Kontynuując temat, który przed chwileczką omawiałem, wszystkie warianty będą następnie rozpatrywane na posiedzeniu komisji oceny przedsięwzięć inwestycyjnych. Wariant preferowany zostanie wskazany na podstawie analizy wielokryterialnej, która będzie elementem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta, wydana przez RDOŚ w Krakowie, wskaże ostateczny wariant przebiegu sądeczanki. Jeżeli nie będzie zastrzeżeń na posiedzeniu KOPI, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie mógł zostać złożony w II kwartale 2021 r. Będzie to kluczowy proces w przygotowaniu tej inwestycji. Istotne jest to, aby decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była ostateczna. Dzięki temu będziemy mieli przesądzony wariant i prace będą mogły być prowadzone bez przeszkód. Jak wspomniałem wcześniej, to zadanie budzi duże zainteresowanie społeczne i może się zdarzyć, że na etapie konsultacji publicznych w ramach postępowania prowadzonego przez RDOŚ mogą pojawić się liczne stanowiska. Co więcej, osoby niezadowolone z przyszłego wariantu mogą się odwołać od decyzji RDOŚ do GDOŚ, co może mieć istotny wpływ na przyszły harmonogram dotyczący przygotowania i realizacji tej inwestycji. Uśmiecham się tu do państwa parlamentarzystów, do wszystkich tych, którym zależy na budowie sądeczanki, aby rozmawiali państwo ze społeczeństwem i uczulali, że odwołania powodują przesunięcie realizacji tej inwestycji.

Tutaj jest prośba do państwa parlamentarzystów o aktywność, o rozmowy z samorządami, ze społeczeństwem i uczulanie co do tego, że inwestycja ta będzie realizowana wtedy, kiedy dojdziemy do wariantu, który uzyska ostateczną decyzję środowiskową. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy, które już są realizowane, to w październiku br. została podpisana umowa na zaprojektowanie i zbudowanie tzw. łącznika brzeskiego, to jest północna część odcinka Brzesko - Nowy Sącz o długości 3 km. Koszt prac wyniesie blisko 100 mln zł. Dziękuję bardzo.

Pytanie: Jaka jest aktualnie liczba środowiskowych domów samopomocy, o ile wzrosła ta liczba od 2016 r., jaka jest aktualnie liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy i ile osób aktualnie z nich korzysta? Dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Domy samopomocy odgrywają bardzo istotną rolę w procesie społecznym, jakim jest udział osób niepełnosprawnych w życiu mieszkańców danego powiatu. Domy samopomocy stanowią sieć wsparcia osób niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi.

W związku z powyższym mam pytanie. Panie ministrze, wiemy, że w roku 2015 tych instytucji w skali kraju było 760.

Dziękuję. Dziękuję panu posłowi.

O udzielenie odpowiedzi proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej pana ministra Stanisława Szweda.

Bardzo dziękuję państwu posłom za to pytanie, bo temat jest bardzo ważny.

Są to placówki typu dziennego, które mogą organizować również krótkoterminowe pobyty całodobowe.

Warto też przypomnieć, że mamy cztery typy środowiskowych domów samopomocy. Typ A - dla osób przewlekle psychicznie chorych. Typ B - dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym, a także dla osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Typ C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia psychiczne.

To jest ważne poszerzenie zakresu działania, bo wiemy, że takich osób nam przybywa. 2 lata już, 3 lata już takie domy też funkcjonują. Teraz przechodzę do konkretnych pytań. Z roku na rok. W roku 2016 było 779 ŚDS-ów, w roku 2019, bo takie mamy na dzisiaj dane - 830, czyli w tym okresie przybyło 51 nowych ośrodków.

Warto oczywiście jeszcze raz przypomnieć, że prowadzenie i rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym zarówno przez gminy, jak i przez powiaty. Co też jest ważne, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej co roku dokonuje podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki te są przekazywane w zależności od zapotrzebowania.

Bardzo proszę, pani poseł. Pani Marszałek! Bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Tu już pan minister wspomniał o działalności ŚDS-ów w czasie pandemii. Wiemy, że sytuacja jest trudna. Ona też jest trudna w środowiskowych domach samopomocy. O tę sytuację chciałam zapytać.

Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Oddaję głos panu ministrowi. Bardzo proszę. Dziękuję za to dodatkowe pytanie, bo to, myślę, bardzo ważna kwestia związana z okresem pandemii.

Jednocześnie ze środowiska osób, które korzystają z tej pomocy, ale również ze środowiska samych pracowników płynęły sygnały, że to rozwiązanie jest bardzo niekorzystne dla podopiecznych. Stąd na następnym etapie już wprowadziliśmy możliwość uruchomienia zarówno ŚDS-ów, jak i klubów.

Kolejna kwestia to była kwestia zapewnienia finansowania działalności w trakcie zawieszenia ich działalności.

Oczywiście na bieżąco były też wytyczne dla środowiskowych domów samopomocy. Warto też powiedzieć, że przekazywaliśmy również środki dezynfekcyjne. To wszystko były działania. Bardzo dobrym działaniem, które miało miejsce, była kwestia wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego. On też dotyczył ośrodków wsparcia, w tym środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej. Jeżeli dorosła osoba niepełnosprawna uczęszczała na te zajęcia, a nie mogła [[Dzwonek]] bezpośrednio uczestniczyć, to ich opiekunowie mogli mieć przyznany dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Informacja bieżąca. Przypominam, że na obecnym posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzona informacja w sprawie stanu polskiej gospodarki i finansów oraz sytuacji przedsiębiorców z takich branż jak turystyka, hotelarstwo, gastronomia, targowa i konferencyjna, taksówkarska i inne w dobie pandemii COVID-19, o której przedstawienie wnosił Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni. Przypominam również, że przedstawienie uzasadnienia wniosku przez posła przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 5 minut. Wystąpienia posłów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty. Na zakończenie dyskusji głos zabierają kolejno przedstawiciel wnioskodawców oraz przedstawiciel Rady Ministrów. Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a wystąpienie przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 5 minut. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie wystąpienia przedstawiciela Rady Ministrów. Czas przeznaczony na rozpatrzenie punktu: Informacja bieżąca nie może być dłuższy niż 90 minut. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców panią poseł Marię Małgorzatę Janyską. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wczoraj w tej Izbie padło wiele prawdziwych i gorzkich słów o budżecie na kolejny rok, o budżecie, który zamiast w tej trudnej sytuacji gospodarczej luzować reguły fiskalne, niestety luzuje stabilność finansów publicznych, a jednocześnie wprowadza nowe obciążenia. Wiele gorzkich słów padło o wydatkach, które są finansowane z ciężkiej pracy przedsiębiorców, podatników i przeznaczane niestety wciąż również na polityczną propagandę i umacnianie władzy. Wiele z tych wydatków okazało się ważniejszych niż systemowa pomoc dla przedsiębiorców, która zapewniłaby, że po okresie kryzysu wrócą oni na ścieżkę rozwoju. Dzisiaj, proszę państwa, trzeba mówić o wszystkich ludziach, którzy składają się na ten budżet, o wszystkich przedsiębiorcach z takich branż jak turystyka, hotelarstwo, gastronomia, targowa, konferencyjna, taksówkarska i z nimi związanych, bo to państwo wielu tym ludziom pod rządami PiS-u zmarnowało przez wiele miesięcy dorobek. Najważniejsze były wybory, światopoglądowe sprawy i wyprowadzanie kobiet na ulicę. Ci przedsiębiorcy to są ofiary politycznych targów tej władzy, a władza powinna w tym czasie wzmacniać i stabilizować gospodarkę i finanse publiczne, żeby zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczne, które z kolei jest podstawą możliwości zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego.

W październiku zamrożono branżę gastronomiczną i związane z nią branże. Premier obiecał, że pomoc będzie natychmiastowa. Dzisiaj, proszę państwa, jest 16 grudnia i mam pytanie: Ilu przedsiębiorców otrzymało już, po prawie 2 miesiącach, pomoc? Śmiem twierdzić, że zero, dlatego że dopiero wczoraj prezydent podpisał tę ustawę. A 10 i 15 grudnia upłynął termin opłacenia składek za listopad, zaś 30 listopada upłynął termin złożenia wniosków o umorzenie danin ZUS-owskich, upłynął, zanim przepisy weszły w życie, bo tak się działa w państwie PiS. Pytam także, czy wiecie, ile firm z branży targowej nie otrzyma żadnego wsparcia z tarczy 6.0. Bo to jest prawie 90%. Bo sprawiliście, że przyjęty jest tylko jeden numer kodu dotyczący organizatorów targów, a reszta - nie. Mówiąc o pokrzywdzonych, o ofiarach lockdownu, opowiadamy o konkretnych osobach, o tych, które jeszcze nie podniosły się po wiosennym lockdownie ze wszystkich zobowiązań, a już stanęły przed kolejnymi. Wielu już straciło wiarę i możliwość odbudowania swoich firm, tak jak pan Jarosław, restaurator z Wrześni, który wraz z całą rodziną przez kilkadziesiąt lat budował, rozwijał i prowadził swój biznes, ale nie dał rady czekać, poddał się i kilka dni temu odebrał sobie życie, bo państwo nie zdążyło. Czy rząd w ogóle ma wiedzę o aktualnej sytuacji i prognozach odnośnie do najbliższej przyszłości, skali możliwych likwidacji działalności, upadłości i nastrojów inwestycyjnych? Czy rząd w ogóle ma przygotowane rozwiązania systemowe i długoterminową strategię? Czy zajął się wsparciami, które są niezbędne, takimi jak np. okresowe obniżenie VAT-u na usługi zagrożonych branż, obniżenie PIT-u, odroczenie płatności innych danin, kosztów należnych Skarbowi Państwa, pobudzenie decyzji konsumenckich w ramach strategii wsparcia i promocji solidarności? Tym się zajmują obywatele, ale o rządzie nie słyszałam. Czy np. myślał również o tym, że trzeba byłoby zwolnić okresowo z podatku bankowego aktywa dedykowane akcji kredytowej dla przedsiębiorców? Czy nie zauważacie także, że rozwiązania, które byłyby systemowe, rozwijające, rozszerzające, powinny być w ustawach, a nie w rozporządzeniach?

Oczywiście wiem, powiecie, że macie w rozporządzeniach takie możliwości. Ale możliwość w rozporządzeniu to nie jest systemowe rozwiązanie, to jest władztwo urzędnicze, a władztwo urzędnicze jest zawsze niesprawiedliwe i nie można liczyć na to, że nie będzie różnicowało przedsiębiorców, zwłaszcza za waszej władzy, bo będziecie różnicować przedsiębiorców, jeśli dostaniecie to władztwo urzędnicze, tak jak różnicujecie samorządy, jeśli chodzi o otrzymywanie środków na przetrwanie tego całego kryzysu gospodarczego.